Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Daniela Milewskiego i Łukasza Schreibera. Protokół i listę mówców prowadzić będzie poseł Łukasz Schreiber. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Informuję, że dziś odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia o godz. 12. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego rozpocznie się dziś o godz. 12 lub po zakończeniu głosowań w wypadku ich opóźnienia. Dziękuję. Wysoki Sejmie! Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożyły dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu ustawy. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski: - w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 2248, - w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 2249. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest to, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy zawarty w druku nr 2212 do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania, bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Wniosek ten poddam pod głosowanie. Jego odrzucenie będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Zdrowia. Poseł Marek Sowa, klub Nowoczesna. Czas na zadanie pytania ustalam na 1 minutę.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Można powiedzieć, że przedstawiciele obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zrealizowali najważniejszy priorytet, przed jakim stoimy, dotyczący naprawy systemu ochrony zdrowia.

Rząd w tej sprawie przez 2 lata nie zrobił dokładnie nic. Chciałbym zapytać wnioskodawców, jakie priorytety w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane z tytułu zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia. Jednocześnie chcę powiedzieć, że Klub Poselski Nowoczesna w pełni popiera przejście od razu do drugiego czytania. Dziękuję panu posłowi. W tej chwili pytanie zadaje pan poseł Marek Hok, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Wysoka Izbo! Dziękuję przedstawicielom inicjatywy obywatelskiej za zebranie w sumie pod dwoma projektami poprawiającymi jakość opieki zdrowotnej, jej dostępność dla pacjentów, jakość pracy fizjoterapeutów, lekarzy, ratowników, pielęgniarek ponad 400 tys. podpisów. Skoro jest takie poparcie, to postanowiliśmy złożyć wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania. To jest test wiarygodności intencji szczególnie rządzących.

Jeżeli większość rządząca jest zdeterminowana, by zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia w Polsce, skrócić kolejki i zwiększyć dostępność, [[Dzwonek]] zagłosuje za niezwłocznym przejściem do drugiego czytania. Było pytanie skierowane do przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! Obecni i Przyszli Pacjenci! Mam dla was złą informację. Nie jesteście nieśmiertelni. i tak jak my, statystyczni Polacy, będziecie umierać. Tak, będziecie umierać 5 lat wcześniej niż obywatele państw zachodniej Europy, którym rządzący starają się zapewnić odpowiednie warunki leczenia. Wyobraźcie sobie człowieka, który zawsze był zdrowy i miał się dobrze. Nagle omdlał, nie wiadomo, co się wydarzyło. Nigdy nie sądził, że go to spotka, jakaś choroba, jakaś słabość, a teraz leży i czeka na karetkę. Każda sekunda czekania na karetkę wydaje się wiecznością. Przychodzą myśli: Czy ona przyjedzie? Czy będzie sprawna? Czy nie zabraknie ratowników medycznych? Czy zapracowana i przemęczona pielęgniarka zdąży wezwać lekarza? Czy będzie mógł przyjść? Czy przyjdzie? Czy będą leki? Myśli się kłębią. Przerażenie narasta.

to zobaczymy, że to ten statystyczny Polak, to ty. To możesz być ty. Ty, czekający w kolejce do gabinetów, w których może zabraknąć lekarzy, bo np. posłuchali rady posłanki Hrynkiewicz i wyjechali za granicę albo z powodu wieku emerytalnego zaprzestali pracować zawodowo. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie! Słuszny protest medyków, czyli fizjoterapeutów, elektroradiologów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów, logopedów, dietetyków, a nie tylko rezydentów, jaskrawo udowodnił katastrofalną sytuację w ochronie zdrowia zaniedbywanej przez wszystkich rządzących od chwili transformacji ustrojowej. Jak dotąd żaden rząd, podkreślam, żaden rząd nie potrafił podjąć radykalnych decyzji w zakresie zapewnienia godnych warunków leczenia Polaków. Mimo głoszonych przez wszystkie partie haseł wyborczych, że sprawa zdrowia obywateli będzie traktowana jako pierwszorzędna, poza rosnącą biurokracją prawie nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie! Stoję teraz przed wami, nie tylko będąc przedstawicielem polskiej służby zdrowia, ale przede wszystkim reprezentując społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, której konstytucja w art. 68 zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. I pytam was o tę dostępność: Gdzie ona jest? Czy ona jest realna? Jeśli nie uświadomimy sobie, że aktualnie wydajemy na ochronę zdrowia. Proszę państwa, proszę o ciszę. A pana przedstawiciela proszę, żeby pan odpowiadał na pytanie, konkretne pytanie posła Sowy. Proszę odpowiedzieć na pytanie.

Obowiązkiem marszałka Sejmu jest pilnowanie, żeby mówca mówił na temat i do rzeczy, więc zwracam panu uwagę. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie! Jeśli nie uświadomimy sobie. Aktualnie wydajemy na ochronę zdrowia 4,67% PKB, a niezbędne minimum minimorum rekomendowane przez OECD to prawie 7% PKB. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie! Nasz obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pod którym podpisało się prawie 160 tys. Polaków, zawiera postulat niezwłocznego podjęcia procesu podwyższania corocznych nakładów budżetowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, aby docelowo w roku 2021 i następnych osiągnęły one wysokość 6,8% PKB, a w roku bieżącym - 5,2% PKB. W naszym obywatelskim projekcie ustawy proponujemy przyjęcie zasady, iż środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na opiekę zdrowotną na dany rok w porównaniu z rokiem poprzednim w pierwszej kolejności przeznaczane są w formie dotacji przekazywanej do funduszu na opłacenie świadczeń opieki zdrowotnej. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie.

Przedstawiam państwu obywatelski projekt ustawy. pod którym podpisało się w ciągu 2 tygodni prawie 150 tys. Polaków chcących, by zapewniono im konstytucyjnie zagwarantowaną opiekę zdrowotną. W imieniu wszystkich pacjentów i tych, którzy zaniemogą, oraz pracowników opieki zdrowotnej wnioskuję o rozpoczęcie prac nad uchwaleniem przedstawionego przez nas projektu ustawy, którym można pomóc uzdrowić chory system ochrony zdrowia. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie! Przyszedł czas na podziękowania. Pilna wizyta u kardiologa dziecięcego - za 4 miesiące. Dziękujemy politykom. Oczekiwanie na diagnozę raka piersi - jedynie 37 tygodni. Dziękujemy politykom. Oczekiwanie na rehabilitację na oddziale rehabilitacji - 12 miesięcy, a w zakładzie rehabilitacji leczniczej - 7 miesięcy. Dziękujemy politykom. Najmniej w Europie personelu medycznego na 1 tys. mieszkańców. Dziękujemy politykom. 14 zł za godzinę ratowania ludzkiego życia. Dziękujemy politykom. Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia. Szanowni pacjenci zgromadzeni w tej Izbie! Decyzja zależy od was. Prędzej czy później też zostaną naszymi pacjentami. Macie szansę przedłużenia życia sobie, swoim rodzicom, przyjaciołom i nam wszystkim - waszym wyborcom. Apeluję do państwa: nie pozwólcie umierać Polakom 5 lat wcześniej niż obywatele państw Europy Zachodniej. Pan w tej chwili ma wystąpienie, a nie odpowiada na pytanie, więc proszę pana, żeby pan odpowiedział na pytanie posła. Apeluję do państwa: nie pozwólcie umierać Polakom 5 lat wcześniej niż obywatele państw zachodniej Europy. Nie pozwólcie na poniżanie stojących w kolejce pacjentów, nie pozwólcie na deptanie godności ludzi ratujących życie innych. Za chwilę nie wytrzymamy łatania dziur naszym kosztem i coś naprawdę wybuchnie, ale wtedy będzie za późno. Poprzyjcie obywatelską ustawę - to wszystkim wam i nam wyjdzie na zdrowie.

Ja streszczam to pytanie. W związku z tym, proszę państwa. Ten wniosek poddam pod głosowanie. Jego odrzucenie będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Zdrowia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 2212, bez odsyłania do komisji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji Zdrowia. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Informacja ministra zdrowia o wynikach rozmów z lekarzami rezydentami oraz planach rządu związanych z kryzysem kadrowym w polskim systemie ochrony zdrowia, zgłoszony przez Klub Poselski Nowoczesna, Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie wejść policji do siedzib kobiecych organizacji pozarządowych dzień po „czarnym wtorku”, zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, - Informacja ministra infrastruktury w sprawie realizacji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina, zgłoszony przez Klub Poselski Kukiz’15,

Informacja prezesa Rady Ministrów na temat oficjalnej wizyty w Polsce prezydenta Turcji pana Recepa Tayyipa Erdogana, w szczególności powodów, dla których Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które po autorytarnej próbie przebudowy Turcji przyjmuje prezydenta Erdogana, oraz charakteru polskiej polityki zagranicznej względem Turcji, zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, - Informacja ministra - koordynatora służb specjalnych w sprawie roli ministra przy wyborze kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgłoszony przez Klub Poselski Nowoczesna.

Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji o wynikach rozmów z lekarzami rezydentami. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji w sprawie obwodnicy Szczecina. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację ministra infrastruktury, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym powołania Komisji Śledczej. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji w sprawie wizyty prezydenta Turcji.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację ministra - koordynatora służb specjalnych w sprawie roli ministra w tej sprawie, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2228. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2228, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2150.

Wysoka Izbo!

Jak rząd zamierza temu przeciwdziałać? Czy pani minister Elżbieta Bojanowska chciałaby odpowiedzieć na to pytanie? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2150, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2241-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Piotra Babinetza o przedstawienie tego sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Połączone komisje: Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Spraw Zagranicznych pracowały wczoraj nad zgłoszonymi poprawkami. W efekcie komisje rekomendują głosowanie przeciwko wnioskowi o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz głosowanie za przyjęciem pięciu poprawek do projektu ustawy. Oczywiście komisje też rekomendują przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję panu posłowi. Nad wnioskiem mniejszości i poprawkami będziemy głosować w pierwszej kolejności, ale w pierwszej z tej pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Wysoka Izbo!

Nie zgadzamy się na to. Nie zgadzamy się na to, aby wydawać rocznie 6 mln na stanowiska dla kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy państwo wiecie. Gdyby pan wiedział, toby pan takich głupot nie opowiadał. Instytut polsko-ukraiński jest nam bardzo potrzebny, szczególnie że są teraz bardzo złe stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą. Jest to nam potrzebne.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Pytanie zadaje poseł Marek Sowa, klub Nowoczesna.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym w sposób szczególny zwrócić się do posłów PiS-u z Małopolski. W tej poprawce proponujemy zmienić siedzibę instytutu z Warszawy na Tarnów. Jest wiele powodów, aby siedziba była właśnie w Tarnowie. Tarnów to najbardziej węgierskie miasto w Polsce, jeśli tak można powiedzieć, z tytułu przyjaźni, która w sposób oczywisty tam jest - towarzystwo przyjaciół Węgier funkcjonuje od 1956 r., ludzie mają nawiązaną współpracę. Felczak był osobą bardzo mocno związaną z Krakowem, z Małopolską. Po uwolnieniu był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spoczywa na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił.

Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

Sejm poprawkę przyjął.

Wysoka Izbo! Kiedyś, za czasów słusznie minionych, mieliśmy instytut przyjaźni polsko-radzieckiej. Teraz, na wzór tego, państwo, idąc cały czas w tym kierunku, z wielki sentymentem do PRL-u, powołujecie instytut przyjaźni polsko-węgierskiej. Doskonale rozumiem, że dla PiS-u współpraca z rządem Orbána ma zasadnicze znaczenie.

Chodzi o instytucję, która obsadza dwie rady, bo krajową i zagraniczną.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął.

Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o współpracę w regionie Grupy Wyszehradzkiej, potrzebujemy trwałych ram instytucjonalnych. Już w październiku zgłosiłem się do pana marszałka z inicjatywą, która jest odpowiedzią również na inicjatywę Węgrów z Jobbiku z tamtejszego parlamentu, by ustanowić stałe zgromadzenie parlamentarne państw Grupy Wyszehradzkiej, dlatego że jeśli chcemy tę współpracę w regionie Europy Środkowej, Europy centralnej zacieśniać, to potrzebujemy instytucji, które będą miały wielostronny charakter w gronie tych czterech państw, może poszerzanym o kolejne, a nie tylko instytutów dwustronnych. Potrzebujemy intensywnej wymiany studenckiej, potrzebujemy zintensyfikowania takich projektów, jak chociażby wspólna telewizja czy wspólny przekaz dla wszystkich państw regionu Europy Środkowej i o to serdecznie ponownie apeluję. Dziękuję panu posłowi. Informuję pana posła i Wysoką Izbę, że od kilku lat trwają starania o utworzenie zgromadzenia parlamentarnego Grupy Wyszehradzkiej.

Pytanie zadaje pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, klub Platforma Obywatelska.

Panie i Panowie Posłowie! Podczas posiedzenia komisji otrzymywaliśmy bardzo mętne tłumaczenia ze strony przedstawicieli rządu, dlaczego właśnie musi powstać taki instytut, takiej rangi, podporządkowany prezesowi Rady Ministrów. Wśród wielu tłumaczeń było i takie, że chodzi tu o zobowiązania i umowę polsko-węgierską. Tak więc rozumiemy, co otrzymał pan premier Orbán od rządu polskiego - instytut, który właściwie będzie jakąś taką czapą nad formami współpracy. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co Polska otrzymała od pana premiera Orbána.

Tutaj o głos prosi pan minister Dworczyk, który kieruje Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wysoka Izbo! Pozwolę sobie przypomnieć, że pani pytała o bardzo szczegółowy zapis dotyczący statutu fundacji powołanej na Węgrzech, i rzeczywiście na pytanie dotyczące tego konkretnego szczegółu nie byłem w stanie na posiedzeniu komisji odpowiedzieć, ale informowałem panią przewodniczącą oraz całą komisję, że będą to dwie siostrzane instytucje, że jeśli chodzi o środki finansowe, to te, które zostały przewidziane na Węgrzech na funkcjonowanie tej instytucji, to jest kwota zbliżona do 5 mln zł, czyli budżet podobny do budżetu, którym będzie dysponował instytut, który właśnie powołujemy. Dziękuję panu ministrowi. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2241, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji, który poddam pod głosowanie.

Wysoka Izbo!

Słowami pani poseł Bartuś zobowiązaliście się z tej mównicy, więc pytam: Kiedy kolejny raz zajmiecie się państwo tą sprawą? Wysoki Sejmie! Powraca pytanie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Skalę hipokryzji w tej sprawie pokazuje fakt, że to przecież posłowie Prawa i Sprawiedliwości domagali się tego wyroku. Wyrok zapadł w październiku 2014 r. Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL, pan minister Kosiniak, zostawił gotową ustawę i pieniądze w budżecie na 2016 r., żeby zrealizować ten wyrok. Minęły ponad 2 lata, przemilczacie to, uciekacie od tych pytań, nie wykonujecie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ludzie zaczęli dochodzić swoich praw przed sądami. Sądy zasądzają te świadczenia, co tylko potwierdza, że tym ludziom się to należy. Kiedy zatem zaczniecie szanować prawa osób niepełnosprawnych i zrealizujecie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego przecież sami się domagaliście? O głos prosi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Co roku uchwała zobowiązuje rząd do przygotowania informacji, w jaki sposób rząd, ministerstwa, urzędy centralne realizują postanowienia karty. Zawiera ona opisy działań zrealizowanych, kontynuowanych lub podjętych w 2015 r. i 2016 r. przez ministerstwa i urzędy w ramach merytorycznych kompetencji i ustawowych uprawnień w zakresie realizacji praw określonych w sejmowej uchwale.

W grudniu 2017 r. komisja bez głosów sprzeciwu przyjęła informację rządu o realizacji postanowień karty w 2016 r. Informacja została przygotowana na podstawie informacji zebranych w poszczególnych ministerstwach i urzędach. Opisuje podjęte działania, opisuje fakty. Zdziwiony jestem, że poseł Platformy Obywatelskiej zgłosił sprzeciw wobec przyjęcia informacji o działaniach podjętych przez rząd. Oczywiście krytycznie podchodzimy do realizacji praw osób niepełnosprawnych za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, natomiast informacja została przygotowana, jak wszystkie poprzednie. Od 20 lat Sejm co roku przyjmuje informację o realizacji postanowień karty. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie sprawozdania w tym brzmieniu, które przyjęła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji zawartej w druku nr 855, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji, który poddam pod głosowanie. Jego odrzucenie będzie oznaczało, że Sejm informację przyjął do wiadomości. Wysoka Izbo!

Ale ja znowu zadam pytanie o zobowiązania sprzed 2 lat. Jednym z celów tej karty jest zabezpieczenie społeczne, godne zabezpieczenie społeczne. Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł. Przez te 2 lata nie drgnął nawet o złotówkę, więc pytam o rzeczy, do których państwo się zobowiązaliście. Zobowiązaliście się państwo do tego, że wyrównacie świadczenia, że wyrok będzie wykonany w momencie, kiedy usprawnicie orzecznictwo. Tylko przypominam pani poseł, państwu, że mówimy o działaniach podejmowanych w roku 2016.

W ciągu ostatniego 1,5 miesiąca roku 2015 w 6 tygodni waszych pierwszych rządów zdążyliście uderzyć w edukację włączającą niepełnosprawne dzieci, uderzyliście w służbę cywilną, wyrzucając preferencje zatrudniania osób niepełnosprawnych, wyrzuciliście do kosza wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o który sami tak skrupulatnie zabiegaliście, a w roku 2016 wasz prezes Kwiatkowski zaczął rozsadzać swoje kwiatki. Maleńkim kwiatkiem było wybranie nowego logo funduszu rehabilitacji, pan prezes Kwiatkowski wybrał kwiatek, ale grubszy kwiatek, który wciąż czeka na wyjaśnienie. To umowa, za którą państwowy fundusz rehabilitacji zapłaci 27 mln zł. Pan prezes Kwiatkowski zawarł umowę ze swoim znajomym i chwalił się tym nawet na Facebooku. Fundusz zawarł na 10 lat umowę najmu pomieszczeń, z których najpewniej nigdy nie skorzysta, ale 27 mln zł z kasy państwowego funduszu rehabilitacji zniknie. Co na to rząd Prawa i Sprawiedliwości? Kto rozliczy tę aferę? Głos ma pani poseł Kornelia Wróblewska, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo!

Przeczytam pierwszy punkt karty: najważniejsze działania prowadzące do optymalizacji podjętych przedsięwzięć w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych. Wracamy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pani minister, to państwa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy, którą przyjęła Platforma Obywatelska. Tłumaczyliście, że jak przejmiecie władzę, będziecie razem z nimi, że zrealizujecie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Mieliście 2 lata, minęły 2 lata i ani w jednej, ani w drugiej informacji nie ma absolutnie słowa na ten temat.

Dlaczego nie wprowadzacie dobrych rozwiązań?

Głos ma poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony. Wysoka Izbo!

Ale w kontekście tej sprawy i tej debaty mam pytanie odnośnie do praw osób niepełnosprawnych: Kiedy stosowne komisje sejmowe zajmą się projektem zniesienia aborcji eugenicznej, która dyskryminuje najbardziej bezbronne osoby niepełnosprawne czy potencjalnie niepełnosprawne, czyli dzieci nienarodzone? Wczoraj po raz kolejny komisje się tym nie zajęły, a 800 tys. obywateli podpisało się pod wnioskiem, żeby jak najszybciej znieść aborcję eugeniczną. Dziękuję. Tylko to jest troszkę inny temat, panie pośle. Jak ja mam odpowiedzieć? Pan minister odpowie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Chciałem podziękować posłom, że wykorzystali pretekst do dyskusji o informacji o realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, żeby przypomnieć Wysokiej Izbie o sytuacji osób niepełnosprawnych, o tym, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, o tym, że by mogły realizować swoje prawa, potrzebują wsparcia i pomocy w wielu dziedzinach życia. Jest to na pewno ważna sprawa i na pewno ważne są głosy, które tutaj padły. Natomiast dzisiaj dyskutujemy o informacji o działaniach rządu w 2015 r. i 2016 r., jeśli chodzi o realizację karty w zakresie kompetencji i obowiązków poszczególnych ministerstw. Bardzo się cieszę, że pan poseł Piechota jest krytyczny wobec rządu pani premier, bo to ona rządziła w 2015 r.

Przecież pan poseł doskonale wie, że dotyczy to osób niepełnosprawnych, ale także osób niesamodzielnych z powodu choroby, wieku czy ze względu na inne przyczyny. Jesteśmy w Wysokiej Izbie, musimy wiedzieć, ile osób z tego korzysta i ile to będzie kosztować. I pan poseł jako doświadczony parlamentarzysta doskonale o tym wie. Proszę państwa, długo można by mówić na temat tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił przez 2 lata i porównywać to z tym, co rządy Platformy Obywatelskiej zrobiły przez 8 lat, ale nie jest to temat tej dyskusji.

Pan poseł Sławomir Piechota w trybie sprostowania, tak? Tylko prosiłbym, żeby pan odnosił się do informacji ministra za rok 2016. To przypominanie nam regulaminu jest wysoce niestosowne, wysoce niestosowne. Natomiast pan minister może mnie nie usłyszał, a może mnie nie zrozumiał. Rząd Platformy Obywatelskiej zakończył swoją kadencję w 2015 r. Czy zostawił projekt ustawy? Zostawił. Czy wpisał w projekt budżetu na 2016 r. pieniądze na wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego? A co zaczęli robić przedstawiciele rządu PiS?

Tak? Pan wicepremier Gowin, pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska, pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To pokazuje skalę arogancji. No w roku 2016, kiedy rządził pan prezes Kwiatkowski, który wyprowadził z PFRON-u 27 mln. W roku 2016. A nasz projekt ustawy, który zostawiliśmy w 2015 r., i wpisane do budżetu pieniądze na realizację tego wyroku - gdzie są? W koszu, w zamrażarce, w głębokiej szufladzie. I dlatego uważamy, że już w roku 2015, w ciągu tych kilku tygodni roku 2015, zaczęliście dewastować budowane przez 8 lat podstawy godnego traktowania osób niepełnosprawnych. W ciągu kilku tygodni i kolejnych miesięcy konsekwentnie te podstawy ochrony praw osób niepełnosprawnych są dewastowane.

Proszę bardzo. Proszę o ciszę. Oprócz szeregu działań, które prowadzimy w ministerstwie edukacji na rzecz dzieci, uwaga, ze specjalnymi potrzebami. Na tym m.in. polega mówienie o edukacji włączającej i edukacja włączająca.

Muszę się, proszę państwa, odnieść do tego, o co oskarża mnie pan poseł.

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji zawartej w druku nr 1802, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do trzeciego czytania. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2243-A. Proszę pana posła Piotra Uścińskiego o przedstawienie tego sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Rado Ministrów! Mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2192. Szanowni Państwo! Komisja przeanalizowała te poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie tych poprawek i przyjęcie w całości projektu ustawy. Dziękuję. Nad poprawkami przedstawionymi przez komisje głosować będziemy w pierwszej kolejności. Przypominam, że chodzi o druk nr 2243.

W 1. poprawce do art. 14 ust. 4 wnioskodawcy proponują inne brzmienie części wspólnej dla punktów wymienionych w tym ustępie. Pytanie zadaje poseł Małgorzata Pępek, klub Platforma Obywatelska.

Wysoka Izbo! Poprawka ta dotyczy ochrony lokatorów. Art. 14 ust. 4 ustawy przedstawia, kogo należy szczególnie chronić, a mianowicie kobiety w ciąży, małoletnich, osoby niepełnosprawne, emerytów i rencistów, korzystających z pomocy społecznej oraz osoby bezrobotne. Do tej pory sąd nie mógł wydać orzeczenia o eksmisji dla tych osób, żeby osoby te mogły zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. W ustawie dodano zapis, cytuję: lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych we własnym zakresie. Uważamy, że dodany zapis jest niejednoznaczny i może być interpretowany na niekorzyść lokatorów, którzy powinni być szczególnie chronieni. Dziękuję, pani poseł. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Pytanie zadaje poseł Elżbieta Stępień, klub Nowoczesna. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zwrócić państwa uwagę na stanowienie prawa, bowiem chcecie państwo skreślić art. 24, który jasno mówi: prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu. Zamieniacie państwo ten zapis na następującą treść: sąd może orzec o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wobec osoby, która dokonała zajęcia lokalu z tytułu prawnego, jeżeli przyznanie tego uprawnienia byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione. Szanowni Państwo! Takie zapisy wręcz zachęcają do samowolnych włamań do gminnych lokali. Dziękuję.

Sejm poprawkę odrzucił. Z tą poprawką łączy się poprawka 4. Pytanie zadaje poseł Małgorzata Chmiel, klub Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo!

Macie taką świetną okazję, bo akurat nowelizujemy tutaj tę ustawę, żeby przy okazji i to wyprostować. Najem instytucjonalny prowadzi wprost do bezdomności, ponieważ lokatorzy muszą się zobowiązać, że nie będzie im przysługiwało prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

Proszę.

Sejm poprawki odrzucił.

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Wysoka Izbo! Poprawka nr 5 dotyczy sankcji za niezłożenie przez najemcę deklaracji o wysokości dochodów na żądanie gminy. W takim przypadku zgodnie z projektem gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku. Obecnie ustawa mówi o możliwości podwyższenia czynszu do 3% wartości odtworzeniowej bez uzasadnienia i powyżej 3% w uzasadnionych przypadkach. Proponujemy, aby obniżyć sankcje do 6% wartości odtworzeniowej lokalu, czyli dwukrotnej wartości obowiązującej w ustawie o ochronie praw lokatorów. To i tak będzie dotkliwa kara. My proponujemy, żeby rząd był jednak bardziej łaskawy i przyjął naszą poprawkę. Należy wziąć pod uwagę to, iż nowelizacja, o której mówimy, to zarówno duża zmiana, jeśli chodzi o zarządzanie mieszkaniami komunalnymi, jak i zmiana, która musi się dokonać w mentalności najemców w związku z ciągłym podwyższaniem czynszów [[Dzwonek]] i weryfikowaniem ich zarobków, a także przedstawianiem oświadczeń gminie, jeśli tylko trochę więcej zarobią. Dziękuję, pani poseł.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obowiązek składania deklaracji o dochodach i majątku wejdzie w życie najwcześniej po 2,5 roku od wejścia w życie tej ustawy. Po drugie, jeżeli nie będzie żadnego rygoru składania deklaracji, to nikt tych deklaracji nie będzie składał. Gminy nie dostałyby żadnych instrumentów, jeżeli chodzi o gospodarkę lokalami. To jest drugi argument. I trzeci, jest to uprawnienie, które gmina dostaje, czyli może maksymalnie podwyższyć czynsz do 8%, ale tylko w okresie, w którym ta osoba tej deklaracji nie złoży. Jeżeli ta osoba deklarację złoży, to czynsz będzie wynikał z jej dochodów. A więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, to będzie całe życie płacił podwyższony czynsz. Jest to pewien rygor zmuszający te osoby do składania deklaracji. A więc absolutnie nie rozumiem tutaj stanowiska państwa, które nie pozwala gminom w sposób racjonalny tym deficytowym towarem, jakim są lokale komunalne, gospodarować. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Aldona Młyńczak, klub Platforma Obywatelska. Poprawka 6. dotyczy sposobu obliczania wysokości czynszu w przypadku, kiedy najemca przekroczy kryterium dochodowe, jakie przyjęto w gminie. I tak np. w Warszawie dla jednej osoby kryterium dochodowe wynosi 1900 zł, dla dwóch, trzech, czterech osób mieszkających w jednym gospodarstwie - 1400 zł. Uważamy, że przyjęty algorytm nadmiernie podwyższa czynsze w stosunku do uzyskanych dodatkowych przychodów. Na podstawie wyliczeń według zaproponowanego algorytmu, zgodnie z tabelą przedstawioną przez ministerstwo, wygląda to następująco.

Uważam, że jest to demotywujące i aspołeczne, dlatego wnioskujemy, aby zmniejszyć o połowę kwotę naliczanych [[Dzwonek]] czynszów bez takich drastycznych podwyżek, aby opłacało się najemcom. Dziękuję bardzo. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw?

Wysoka Izbo! Mając na uwadze, iż przedstawiona nowelizacja ma pozwolić samorządom bardziej racjonalnie i efektywnie gospodarować komunalnym zasobem mieszkaniowym, co w długotrwałej perspektywie powinno jednak przyczynić się do udzielenia pomocy mieszkaniowej szerszej grupie mieszkańców, Platforma Obywatelska będzie głosowała za przyjęciem projektu ustawy. Aczkolwiek uważamy, że istota zmian zawsze tkwi w szczegółowych zapisach, stąd też nasze poprawki, a także sugestia, aby w dalszych pracach nad ustawą zmienić algorytm do obliczania wysokości czynszu na bardziej korzystny dla najemców, zmniejszyć maksymalne sankcje za niezłożenie oświadczenia w sprawie dochodów, a także zmienić zapisy najmu instytucjonalnego. Głos ma poseł Anna Milczanowska, klub Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać pana wiceministra, czy prawdą jest, że samorządy terytorialne czekają na tę ustawę, że zwiększamy sześciokrotnie kwotę na budowę mieszkań socjalnych, komunalnych, noclegowni, mieszkań tymczasowych do kwoty 6 mld zł, że chcemy oddać takim sposobem 170 tys. nowych mieszkań, że są oczekiwania, aby - i takie rozwiązanie stosujemy również w tej ustawie - była możliwość współfinansowania budowy nowych budynków mieszkalnych, socjalnych z pieniędzy unijnych, i że na to wszystko czeka polski samorząd.

Wysoka Izbo!

Dlatego wprowadzamy rozwiązania, które dają możliwość podwyższania czynszu osobom zamożnym, bo te mieszkania nie są dla osób zamożnych, one są dla tych, którzy czekają w kolejce i spełniają kryterium dochodowe. Nie chcemy tych osób zamożnych wyrzucać z tych mieszkań, ale niech one płacą wyższy czynsz. Wyższy czynsz daje wyższe dochody gminom, co pozwoli więcej tych lokali zbudować. Są nowe rozwiązania, jest grant 20-procentowy, jest możliwość budowania pomieszczeń tymczasowych, nie ma eksmisji na bruk. To są rozwiązania, na które samorządy czekają. Zastrzeżenia, które państwo składają, oczywiście są dyskusyjne, bo każde podwyższenie czynszu jest niewygodne. Ale musimy pamiętać, że przede wszystkim musimy chronić tych, którzy czekają w kolejce, te 0,5 mln osób, które mają niskie dochody i nie stać ich na płacenie czynszu wyższego niż czynsz komunalny. Proszę. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2243, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Przypominam, że komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2237. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2237, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W trakcie drugiego czytania do projektu uchwały zgłoszono poprawkę.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 2205. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszoną do projektu uchwały poprawkę. Wnioskodawcy, przypominam, proponują w niej dodanie akapitu dotyczącego podwojenia unijnych dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło poprawkę, aby polscy rolnicy mieli podwojone dopłaty unijne. Jest to wyjście naprzeciw posłom Prawa i Sprawiedliwości. Tak, moi drodzy, bo to wy w czasie kampanii wyborczej obiecywaliście polskim rolnikom, że jak dojdziecie do władzy, to podwoicie dopłaty unijne.

Możecie to nazwać hipokryzją, dwulicowością albo rozdwojeniem jaźni. Proszę bardzo, wybór należy do was. Pytanie: Czy poprzecie tę poprawkę [[Dzwonek]] i kiedy zrealizujecie wasze obietnice, że podwoicie dopłaty dla polskich rolników? Wysoka Izbo! Akuratnie jak PSL dba o polskie rolnictwo, to teraz widzimy. Aczkolwiek takie pytanie powinno tutaj paść, a właściwie odpowiedź ministra powinna paść. Może się okazać, że ta uchwała będzie równie pusta jak ta uchwała z 2012 r. My tutaj jako parlament wspieramy ministra, minister będzie negocjował, a wczoraj minister mówi o pewnym wyrównaniu dopłat. Czyli jakim pewnym? Ono powinno być chociażby na poziomie dopłat niemieckich, a nie mniejsze. A może się okazać, że ono będzie tak niepewne, jak i poprzednia koalicja.

Wczoraj długo debatowaliśmy o nowych negocjacjach w sprawie wspólnej polityki rolnej. W kampanii wyborczej, potem w swoim exposé wasz jeden premier, drugi, a także posłowie wielokrotnie z tej mównicy grzmieli, że polscy rolnicy nie mogą być w Europie tak nierówno traktowani. Ale wciąż nie rozumiemy, jaki jest wasz cel w tym nierównym traktowaniu. A więc jeżeli pan minister pozwoli i nie umie sam sobie postawić celów, to ja przypomnę, jakie cele stawia przed panem klub Nowoczesna. Polska miała najwyższy budżet na rozwój w II filarze wspólnej polityki rolnej i tym liderem musi pozostać.

Polska, ale też Łotwa Rumunia, Bułgaria i Węgry zwiększały swoje budżety.

Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie! My życzymy rządowi, żeby wynegocjował większe pieniądze niż uczyniła to nasza koalicja. Trzymamy kciuki za polski rząd, żeby ta kwota była wyższa, [[Oklaski]] bo potrzeby polskich gospodarstw są ogromne.

Dlatego ten budżet musi być wyższy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym najpierw podziękować parlamentowi, że taka uchwała będzie podjęta. W poprzedniej kadencji na nasz wniosek, Prawa i Sprawiedliwości, też przyjęto taką uchwałę. Myślę, że w sytuacji, jaka jest, jeśli parlament przyjmie.

Nasz cel jest jasny, cel polityki rolnej na arenie międzynarodowej: równe warunki konkurencji, to, żeby wszyscy rolnicy w Europie mieli równe warunki konkurencji. Jest to całe prawo unijne, prawo żywnościowe dotyczące i GMO, i środków ochrony roślin.

Wy tego nie rozumiecie, dlatego że w Unii Europejskiej pierwsza trudność, jaka jest, panowie, jest taka, że w ostatnich negocjacjach Polsce przysługiwało 21,2 mld euro na dopłaty.

mówię właśnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które brało udział w negocjacjach w 2003 r. - co to znaczy równe dopłaty, jak powstawała koperta krajowa. To nie jest trudne, ale trzeba się wsłuchać i jednak sięgnąć do doświadczeń, chyba że panowie nie macie w tym zakresie świadomości. Koperta powstawała w ten sposób: równe dopłaty, tzn. do pewnego rodzaju produkcji.

Na przykład Włosi mieli 60, Francuzi - też coś koło tego. My mówimy o odejściu od wartości historycznych. Druga sprawa, panowie.

W Polsce jest inny system, system obszarowy. Musicie zrozumieć, że równe warunki konkurencji i wyrównanie dopłat dotyczą poszczególnych rodzajów produkcji.

Chcę panu posłowi powiedzieć - w komisji wielokrotnie o tym mówiono - że jeśli chodzi o finansowanie czy perspektywę finansową, to elementy finansowe, wielkość środków ustalają premierzy, Rada Europejska, i tutaj minister jest tylko doradcą pana premiera, i rząd, natomiast reprezentuje nas w Radzie Europejskiej premier, który w tym zakresie podejmuje decyzje. Jeśli chodzi o pytanie pana Plocke, to nie jest to prawda. Skąd pan wziął te 42 mld euro w poprzedniej perspektywie finansowej? Nie wiem, skąd pan zna te sumy. Powiem panu tak: 9,8 mld było na rozwój obszarów wiejskich.

Tak że w sumie to daje 28 mld.

Dziękuję. Głos w tej chwili zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Robert Telus. Wysoki Sejmie! Chcę również powiedzieć, że dyskusja była bardzo rzeczowa, jeżeli chodzi o tę uchwałę, ale co do tej poprawki, którą wniosło Polskie Stronnictwo Ludowe, chcę powiedzieć, że to jest największa hipokryzja, jaką może pokazywać Polskie Stronnictwo Ludowe, że można.

Chcę przypomnieć: w 2002 r., przed 2004 r. Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kalinowski.

Drodzy państwo, czy pamiętacie, kto negocjował w drugiej perspektywie? Oczywiście, że PSL, minister Kalemba. Oszukał polskiego rolnika, [[Poruszenie na sali]] bo w drugiej turze. I teraz Polskie Stronnictwo Ludowe składa wniosek.

Jaka jest sytuacja w polskim rolnictwie, to jest wasza wina. My w tej chwili musimy robić wszystko. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

PiS nie chce podwojenia dopłat dla polskich rolników. Oszukaliście, wyzyskaliście polską wieś, teraz ją odrzucacie. Szczytem hipokryzji i obłudy było mówienie: poradzimy sobie z ASF-em. Premier Morawiecki rozszyfrował ten skrót, ale z 3 ognisk ASF-u, gdy przejmowaliście rządy, jest 107 ognisk i ASF przekroczył Wisłę. Szczyt hipokryzji, nie poradziliście sobie z ASF-em. Szczyt hipokryzji: obniżymy wszystkim wiek emerytalny. Nie, nie wszystkim po wyborach. Rolnikom podnieśliście z dnia na dzień o 5 lat, zmieniając ustawę pana prezydenta. Szczyt hipokryzji i szczyt obłudy.

Szczyt hipokryzji, szczyt obłudy. Nie chcecie zmieniać polskiej wsi na lepsze. Pytanie zadaje poseł Paulina Hennig-Kloska, klub Nowoczesna. Panie Marszałku! Szkoda, że nie mogłam sprostować wypowiedzi pana ministra, bo pan minister trochę próbuje nam tutaj zamazać obraz. Nie trochę, chyba nawet bardzo.

Część krajów na ten cel przeznacza 10% swojego budżetu w ramach wspólnej polityki rolnej, a my aż 30%.

Głos ma poseł Dorota Niedziela, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Szanowna Izbo! Panie Ministrze! Panie Prezesie! Proszę wziąć do oślej ławki ministra Jurgiela, bo pan prezes krzyczał o tym, że trzeba podwoić dopłaty. Pan minister Jurgiel nie dosyć, że nie ma takich ambitnych celów, nie chce się nawet na nie zgodzić, to jeszcze doprowadził swoim brakiem działania do wystąpienia epidemii ASF-u. W tej chwili będzie nas czekało zabicie 2 mln świń i zlikwidowanie kilkuset gospodarstw, a pan Jurgiel wychodzi tutaj i mówi, że dba o rolników. To hipokryzja. Pan może mówić długo, wiemy o tym, nawet 7 godzin, pan już to robił na tej sali. Boi się pan jechać do Unii i negocjować, dlatego potrzebuje pan wzmocnienia parlamentu w taki sposób, żeby pan mógł się przygotować do porażki. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Wysoki Sejmie! Sprawa dotyczy dopłat rolniczych, więc mam pytanie, czy ktokolwiek na tej sali wie, jak są naliczane dopłaty obszarowe dla rolnictwa, na jakiej podstawie, w jakim systemie. Czy ktokolwiek wie? Nikt nie wie, ponieważ przepisy, które zostały. ponieważ PSL. zgodził się na taki system naliczania dopłat dla polskiego rolnictwa, który nie jest możliwy do przeprowadzenia w ten sposób, o którym oni teraz mówią. Jeżeli system naliczania dopłat według plonu referencyjnego przyjmował 66 euro do 1 t zboża z hektara i jeżeli mówicie, że mamy podwoić płatności obszarowe, to musimy zacząć od tego, że dzisiaj według systemu, na który się zgodziliście, musimy podwoić średni plon zboża z hektara, bo w takim systemie.

Mówiliśmy o równych warunkach konkurencji i o równych dopłatach. A równe dopłaty. Mówiłem też o tym, co to znaczy: równe dopłaty w poszczególnym rodzaju produkcji. Nigdy nikt z polityków Prawa i Sprawiedliwości, z tych, których obserwowałem, nie powiedział o podwojeniu dopłat. Niech pan po prostu nie kłamie.

My obniżyliśmy na 60 lat. Rozumie chyba pan to.

Teraz prowadzimy negocjacje w tym zakresie. I nie jest prawdą to, co powtarzają politycy inni, że nasz rząd nie jest aktywny. Tylko w styczniu spotkałem się z 16 ministrami rolnictwa Unii Europejskiej, podpisaliśmy porozumienie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, podpisujemy porozumienie w ramach krajów bałtyckich, teraz będzie rozmowa z ministrem Francji, już jedna była, natomiast czekamy na wyłonienie ministra Niemiec, żeby zwołać się w ramach Trójkąta Weimarskiego i też wspólne stanowisko przyjąć. Jeśli chodzi o to, co powtarza pan Kosiniak-Kamysz, ceny minimalne - nie ma obecnie w ekonomii w Polsce możliwości wprowadzenia cen minimalnych. Ale jedno muszę tu państwu powiedzieć, wczoraj o tym mówiłem. Bardzo dobry jest program samorządowy PSL-u. A dlaczego? Zdaniem PSL-u. Wywłaszcza on polskich chłopów. W pkt 5 napisano, że PSL będzie wykupywał 10-hektarowe gospodarstwa od rolników i będzie przekazywał do Skarbu Państwa i będzie wydzierżawiał tę ziemię. Dziękuję. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały z druku nr 2205, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2136, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2161.

Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie. Proszę pana posła Jana Dudę o przedstawienie tego sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1424. Połączone komisje na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r. rozpatrzyły 9 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu przez Klub Parlamentarny Kukiz’15. Po dogłębnej analizie przedstawionych poprawek, wysłuchaniu organizacji rolniczych i ekologicznych, które brały udział w pracach nad projektem ustawy od samego początku procedowania, komisje negatywnie opiniują poprawki od 1. do 8. Zaproponowane w projekcie rozwiązania są wystarczające i wykonują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast poprawki 2., 3. i 4. dotyczące ubezpieczeń potencjalnych upraw, wymagałyby zmian innych aktów prawnych. Pozytywnie zaopiniowana poprawka nr 9 zmienia dolną granicę odpowiedzialności karnej z 3 miesięcy do 2 lat za uwolnienie GMO do środowiska w wyniku prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej bez wymaganego zezwolenia. Sprawozdanie połączonych komisji zawarte jest w druku nr 2029-A. Przy okazji dziękuję za włączenie się w prace organizacji rolniczych i ekologicznych, chociaż tu bardzo różnie bywało. Dziękuję ministrowi Szwedzie-Lewandowskiemu oraz jego zespołowi prawnemu za merytoryczny wkład w wypracowanie ostatecznego kształtu projektu. Dziękuję posłom za prawie roczną trudną pracę w podkomisji nadzwyczajnej i w połączonych komisjach ochrony środowiska i rolnictwa. Wysoka Izbo!

Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej dotyczącego zmian w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. d. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Pytanie zadaje poseł Jarosław Sachajko, klub Kukiz’15.

Pamiętam, że dokładnie tak samo pan sprawozdawca był pewien przy pierwszym projekcie ustawy, gdzie był zapis o 3 km.

Głos ma poseł Dorota Niedziela, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czy pan nie wiedział, co mówił, czy pan ich okłamał, że zwiększy pan dopłaty bezpośrednie?

Oczywiście, proszę państwa, przedstawicielem rządu w tym punkcie jest wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

Wysoka Izbo! Chciałem państwa posłów poinformować, że poseł sprawozdawca wprowadził państwa w błąd.

Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Dobrze. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z państwa jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Wysoka Izbo!

Dlaczego uważamy, że dane osób, które będą chciały uprawiać GMO, mają być tajne, mamy je utajniać?

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem poprawki 8., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął.

Wysoka Izbo! Mamy tu kolejny przykład syndromu: bo łgały, więc dostały różnego rodzaju profity. Pan minister Szyszko przygotował ustawę, do której tak naprawdę nie wprowadził żadnych, ale to żadnych poprawek społecznych, które były dla ludzi ważne. Poprawił parę rzeczy, a pominął najważniejsze - społeczne odczucie ludzi, którzy są przeciwko GMO. W 2015 r. rząd Platformy Obywatelskiej i PSL zgłosił nas do Unii Europejskiej jako kraj wolny od GMO.

Głos ma poseł Ewa Lieder, klub Nowoczesna. Szanowny Panie Marszałku! Ten projekt mówi o formalnych warunkach odnoszących się do ewentualnego prowadzenia upraw GMO w Polsce, jednak nie określa, kto poniesie koszty i odpowiedzialność za ewentualne zanieczyszczenia sąsiadujących z nimi upraw tradycyjnych i ekologicznych. Co zamierzacie państwo z tym zrobić?

Prawie zawsze, w 99%. Tak było z Prawem łowieckim. Wszyscy byli niezadowoleni. Robicie to regularnie. Lekceważycie ludzi.

Niestety wiele poprawek, które zgłaszaliśmy, zostało odrzuconych, dlatego nie możemy poprzeć tak dziurawej ustawy. Wysoka Izbo! Marek Sawicki jako minister rolnictwa w 2015 r. zgłosił w Unii Europejskiej Polskę jako kraj wolny od GMO. Wy od tego odstępujecie, dlatego nie popieramy tego rozwiązania. A teraz dwa zdania do pana ministra Jurgiela. Widzę, że pan czyta nasze dokumenty programowe. Upatruję w tym nadziei dla pana, bo jest szansa, że wreszcie będzie program dla polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Proszę dalej z tego korzystać, to na pewno na polskiej wsi będzie lepiej. Prześlemy pełną wersję dokumentów programowych. Pan tak dużo czasu w swoich wypowiedziach poświęca mojemu stronnictwu.

Wysoka Izbo!

Równocześnie jemy to wszystko. Czy prawdą jest, że w tej chwili, żeby wysiać takie nasiona, trzeba mieć zgodę ministra?

że również trzeba zachować bezpieczeństwo środowiska. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2029, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2248, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 409, przeciw - 1, 8 posłów wstrzymało się. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2249) Prezydium Sejmu, na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2249, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę Ogłaszam 5-minutową przerwę.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Pawła Lewandowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Wysoki Sejmie!

W związku z opóźnieniem Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce dotyczącej braku implementacji, dlatego przyjęcie ustawy stało się zadaniem niezwykle pilnym. Dotyczy to także wdrożenia w praktyce przepisów już uchwalonych przez parlament. Poza wdrożeniem przepisów dyrektywy projektowana ustawa będzie stanowić pierwszą w prawie 100-letniej historii polskiego prawa autorskiego w pełni kompleksową regulację działalności organizacji zbiorowego zarządzania. Celem projektodawcy było uporządkowanie polskiego rynku zbiorowego zarządu, wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości oraz uczynienie go bardziej przejrzystym, efektywnym i przyjaznym zarówno dla właścicieli praw autorskich i pokrewnych, jak i dla użytkowników.

Dlatego w praktyce w części organizacji, pomimo że są one stowarzyszeniami uprawnionych, samorządność stała się fikcją, zaś funkcjonujący od lat 90. system zbiorowego zarządu w Polsce ma charakter konfrontacyjny, a nie negocjacyjno-koncyliacyjny. Bardzo ograniczone są też obecnie kompetencje ministra kultury i dziedzictwa narodowego sprawującego nadzór nad organizacjami, co uniemożliwia skuteczne zwalczanie zidentyfikowanych nieprawidłowości. Wdrożenie dyrektywy jest najlepszą okazją do kompleksowego naprawienia tego stanu rzeczy. W Polsce jest potrzeba istnienia rodzimego rynku zbiorowego zarządzania, także jako elementu ochrony rodzimej twórczości, ale musi to być rynek działający efektywnie i według bardziej transparentnych reguł niż dotychczas. Jednym z istotnych elementów ustawy, także w tym kontekście, jest ochrona wykonywania zbiorowego zarządzania na polskim terytorium przez polskie organizacje zbiorowego zarządzania. Unijna dyrektywa pozwala w tym zakresie na utrzymanie istniejącego systemu zezwoleń dla organizacji zbiorowego zarządzania. Umożliwia także wprowadzenie w przypadku zagranicznych podmiotów, które są zainteresowane świadczeniem tego rodzaju usług w Polsce, identycznych obowiązków związanych z rozpoczęciem wykonywania zbiorowego zarządzania jak w przypadku podmiotów polskich, w tym w zakresie uzyskania zezwolenia po spełnieniu określonych kryteriów. Jednocześnie projektowana ustawa zmierza do utrzymania charakteru istniejących organizacji, w których decydujący głos powinni mieć twórcy i artyści wykonawcy, a nie podmioty, których wkład w powstanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych ma charakter finansowy - np. producenci i wydawcy muzyczni - i które prawa autorskie czy pokrewne nabywają od twórców i artystów wykonawców. W tym celu projektowana ustawa oddaje organizacje zbiorowego zarządzania na powrót w ręce ich członków. Podstawowym celem każdego, kto chce zachować bądź ubiegać się o status organizacji zbiorowego zarządzania, musi być zbiorowe zarządzanie ich prawami, wykonywane w sposób staranny, ze szczególnym naciskiem na regularny podział i wypłatę zainkasowanych środków. Stowarzyszenia te mogą oczywiście prowadzić dodatkowo działalność socjalną, kulturalną lub edukacyjną, przy czym musi ona - w zakresie, w jakim jest finansowana z przychodów z praw autorskich i pokrewnych - być prowadzona przede wszystkim na rzecz kategorii uprawnionych reprezentowanych przez organizację i za zgodą tych, z których środków działalność taka jest finansowana. Wszystkie najważniejsze decyzje zapadające wewnątrz stowarzyszenia, dotyczące wynagrodzeń pobieranych na rzecz uprawnionych, muszą być podejmowane na walnym zebraniu członków, a nie - tak jak czasem bywa obecnie - delegowane wąskiemu kręgowi osób zasiadających we władzach stowarzyszenia. Istotne jest umocowanie w ramach organizacji komisji rewizyjnych, których członkowie reprezentujący samych uprawnionych powinni jako pierwsi nadzorować sposób, w jaki ich własna organizacja wykonuje swoje obowiązki wobec nich i wobec ich kolegów.

Podstawową zasadą w tym zakresie będzie równe traktowanie uprawnionych, przestrzeganie terminów i zasad wypłaty środków uprawnionym oraz zasad efektywnego poszukiwania uprawnionych, w przypadku których środki zostały pobrane, ale nie zostały podzielone i wypłacone. To uprawnieni winni wyrazić zgodę na treść dokumentów wewnętrznych, które regulują te zasady, mieć wpływ na wysokość potrąceń dokonywanych przez ich organizację tytułem kosztów wykonywania zbiorowego zarządzania oraz decydować o przeznaczeniu środków na cele inne niż bezpośrednia wypłata. Organizacje nie powinny także mieć prawa do inwestowania nie swoich środków w ryzykowne instrumenty rynku finansowego. Podobnie jak obecnie, podjęcie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania będzie wymagało - jak już wspomniano - zezwolenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ma to na celu zapewnienie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania zbiorowego zarządu oraz ograniczenie nadmiernej liczby organizacji działających na rynku.

Uprawnionych, którzy nie powierzyli praw żadnej organizacji, będzie reprezentować wyłącznie organizacja, która uzyskała status reprezentatywnej. Ponadto organizacje, których zezwolenia się pokrywają, będą zobowiązane do wspólnego zawierania umów z użytkownikami. Dodatkowo w zakresie publicznego odtwarzania wprowadzona zostanie zasada jednego okienka, co oznacza, że użytkownik będzie zobowiązany do zawarcia tylko jednej umowy zamiast czterech lub sześciu, jak obecnie. Rozwiązania te będą istotnym ułatwieniem dla tysięcy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Ustawa zawiera ponadto przepisy usprawniające procedurę zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego. W ślad za dyrektywą ustawa reguluje także zasady udzielania licencji wieloterytorialnych na korzystanie z muzyki w Internecie. Ta część ustawy stanowi literalne wdrożenie dyrektywy, która w tym zakresie dokonała pełnej harmonizacji i powinna być jednolicie wdrożona w całej Unii Europejskiej. Projekt zakłada znaczące rozbudowanie przepisów o nadzorze ministra kultury i dziedzictwa narodowego nad organizacjami zbiorowego zarządzania, poszerzając katalog środków, jakie organ nadzoru może stosować w celu wyjaśnienia i wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości. Ich celem będzie przede wszystkim stosowanie w organizacji działań naprawczych - od miękkich rekomendacji po nakładanie grzywny na osoby winne nieprawidłowości. Dopiero w razie ich bezskuteczności minister będzie mógł zastosować sankcję w postaci cofnięcia zezwolenia na zbiorowe zarządzanie, jedyną przysługującą mu obecnie. Przepisy określają też przeznaczenie środków, jakie pozostały niewypłacone przez organizację, która utraciła zezwolenie w trybie sankcyjnym. Ustawa określi wreszcie - obecnie w żaden sposób nieuregulowane - warunki zarządzania prawami na zasadach komercyjnych przez podmioty niebędące organizacjami zbiorowego zarządzania. Działalność ta będzie miała charakter regulowanej działalności gospodarczej i podlegać będzie rejestracji. W odróżnieniu od organizacji zbiorowego zarządzania niezależne podmioty zarządzające zawsze będą musiały wylegitymować się indywidualnym upoważnieniem do zarządzania konkretnymi prawami. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Głos ma pani poseł Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zgodnie z art. 1, wskazującym zakres regulowanych ustawą spraw, określa zasady: działania organizacji zbiorowego zarządzania oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, tzw. niezależnych podmiotów zarządzających; udzielania zezwoleń na tego rodzaju działalność; nadzoru nad jej wykonywaniem oraz działania Komisji Prawa Autorskiego. Przedłożenie ma charakter dostosowawczy - do prawa Unii Europejskiej - i ma implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania on-line na rynku wewnętrznym z 2014 r. Harmonizacja zasad zbiorowego zarządu w prawie Unii Europejskiej była rozważana od wielu lat. W komunikacie Komisji Europejskiej z 2004 r. wskazywano, że stworzenie rynku wewnętrznego w obszarze praw autorskich i pokrewnych wymaga skutecznych mechanizmów zarządzania tymi prawami, w szczególności w środowisku cyfrowym, w którym wzrasta potrzeba licencjonowania ponadgranicznego, a więc istnienie efektywnego systemu zbiorowego zarządu leży w interesie zarówno uprawnionych, jak i użytkowników. Transponowana dyrektywa szczegółowo reguluje niemal wszystkie aspekty działalności organizacji zbiorowego zarządu, tj. ogólne zasady działania, relacje pomiędzy organizacją a uprawnionymi, zasady członkostwa, strukturę wewnętrzną i władzę, zasady zarządzania przychodami z praw, w tym dokonywania potrąceń od pobranych środków, relacje pomiędzy organizacjami, relacje z użytkownikami, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, w końcu zasady rozstrzygania sporów z udziałem organizacji. W preambule dyrektywy tę kompleksowość legislacji uzasadnia się znaczącymi różnicami w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec członków i podmiotów uprawnionych. Natomiast jako podstawowe cele legislacji preambuła wskazuje zapewnienie koordynacji krajowych przepisów dotyczących warunków podejmowania działalności w zakresie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz ustanowienie wymogów mających zapewnić wysoki poziom zarządzania, zarządzania finansowego, przejrzystości i sprawozdawczości. Zasady ogólne przyjęte przez polską ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w wielu przypadkach są zgodne z kierunkiem wskazanym w dyrektywie. Jednocześnie jej zapisy są zbyt ogólnikowe, a także fragmentaryczne, całkowicie pomijają np. niektóre istotne aspekty zbiorowego zarządu, takie jak np. stosunki organizacji z uprawnionymi czy zasady podziału i wypłaty zainkasowanych środków. W związku z powyższym rząd uznał, że wdrożenie dyrektywy do polskiego porządku prawnego wymaga przyjęcia nowej regulacji zbiorowego zarządu, która znacząco poszerzy zakres regulowanych kwestii oraz uszczegółowi zapisy niektórych istniejących już w praktyce rozwiązań. Wydaje się, że słusznie zdecydowano, że regulacja ta powinna znaleźć się w odrębnej ustawie zastępującej obecny rozdział 12 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przy założeniu utrzymania i rozwinięcia niektórych rozwiązań charakterystycznych dla polskiego systemu zbiorowego zarządu. W wyniku przeprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacji społecznych w sprawie tego projektu wpłynęło 50 stanowisk od organizacji zbiorowego zarządzania, organizacji twórców kultury, izb gospodarczych zrzeszających użytkowników utworów i przedmiotów praw pokrewnych, instytucji kultury, organizacji bibliotekarskich, nadawców telewizyjnych, instytutów naukowych oraz organizacji społecznych i osób fizycznych. Zgłoszone w ramach konsultacji uwagi zostały częściowo przez ministra uwzględnione. Panie Marszałku! Klub Prawo i Sprawiedliwość jest za skierowaniem rządowego projektu o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do dalszych prac parlamentarnych. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

Także ta próba, zwłaszcza że wynikająca częściowo z dyrektywy Komisji Europejskiej, jest próbą, nad którą zapewne należy się bardzo wnikliwie pochylić, próbą, która wymaga chyba bardzo szczegółowego przeanalizowania na forum parlamentu.

Pojawiła się inicjatywa, były konsultacje, sprawdzano ustawodawstwo państw europejskich, więc to było 10 lat. Potem, jak rozumiem, obecny rząd - i dobrze, że się natychmiast zmierzył z tą tematyką. pracował chyba ok. 2 lat. Jest to bardzo trudna, bardzo obszerna ustawa.

Tak naprawdę, to myśmy się dowiedzieli w poniedziałek, że ten projekt jest przedmiotem posiedzenia plenarnego.

Takie jest zdanie mojego klubu. Dlatego też pozwolimy sobie złożyć wniosek o wysłuchanie publiczne i osobiście jestem przekonana - to będzie wniosek do komisji kultury - że komisja kultury poprze ten wniosek.

Tak że z takim wnioskiem o wysłuchanie publiczne zwrócimy się na pierwszym etapie.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dyrektywa, która została nam przedstawiona, rzeczywiście musi być wdrożona. Cieszę się, że rząd podjął takie wyzwanie, by poza dyrektywą pójść dalej i uregulować rzeczy istotne, ważne.

Dlatego myślę, że.

Dużo już zostało zrobione, została napisana bardzo duża ustawa. Dlatego myślę, że twórca z pokorą podejdzie również do poprawek, które mogą się pojawić podczas tych prac, oraz z pokorą i z pewnym szacunkiem dla artystów da możliwość pracy, tak aby to prawo było jak najlepsze. Myślę, że na tym nam wszystkim zależy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. I zapraszam pana posła Krzysztofa Mieszkowskiego z Nowoczesnej. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

To jest bardzo szerokie pole do dyskusji i tę dyskusję oczywiście trzeba podjąć. Bardzo się cieszę z tego, że pan minister i państwo podjęliście to wyzwanie, bo trzeba to wszystko uregulować. Jednocześnie popieram propozycję pani wiceprzewodniczącej Śledzińskiej-Katarasińskiej o wysłuchanie publiczne. Prawdopodobnie przez następne lata będzie bardzo trudno zająć się tym problemem i wrócić do niego, więc jest okazja, żeby to sensownie, dogłębnie przedyskutować, tak żeby nie pominąć nikogo ze środowiska szeroko rozumianych artystów kultury czy instytucji kultury. Jeśli ktoś z państwa chce się zapisać do głosu, to zapraszam, zamknę listę po pierwszym pytaniu. Głos ma pan poseł Józef Lassota, Platforma Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym na etapie pierwszego czytania poprosić pana ministra o to, aby może przedstawił główne postulaty wynikające z tych konsultacji, te, które były lub zostały uwzględnione w stosunku do pierwotnej wersji projektu, jak również te, które nie zostały uwzględnione. Zdaję sobie sprawę, że pewno były także opinie być może sprzeczne ze sobą, ale taka informacja jest niezwykle przydatna dla dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam panią poseł Joannę Fabisiak, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Wdrożenie tej dyrektywy było bardzo oczekiwane przez środowiska twórców.

To dobry pomysł, że będzie wysłuchanie publiczne. Ale najistotniejszą sprawą, tak jak było tu podkreślane, jest sprawa zabezpieczenia twórczości rodzimej, polskiej i zabezpieczenia tych właściwych praw twórców. Na tym nam zależy. Tak jak mówię, wiele środowisk zwracało się z prośbą, aby te sprawy - co będzie oczywiście możliwe w czasie dyskusji - wróciły, aby te wnioski wróciły. I to może jest rzecz najważniejsza.

Zatem ogromna prośba, byście państwo w tym zakresie przedstawili główne postulaty i główne założenia rozszerzenia [[Dzwonek]] tych paragrafów dotyczących działalności Komisji Prawa Autorskiego. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Pawła Lewandowskiego. Dziękuję, panie marszałku, pani poseł, panie pośle. Wysoka Izbo! Żadna z organizacji zbiorowego zarządzania ani żaden z podmiotów, które brały udział w konsultacjach, nie zgłosiły postulatu, że co do zasady ustawa źle reguluje kwestie, które ma regulować. Jeśli zaś chodzi o szczegółowe przedstawienie wszystkich postulatów i nasze odpowiedzi na wszystkie postulaty - bo ja nie wiem, które postulaty mogę uznać za główne, a których nie mogę - to znajduje się to w raporcie z konsultacji, który jest oczywiście załączony do dokumentacji złożonej w Sejmie. Jest on również dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Bo przypominam, że ustawa jest duża, długa, co sami państwo posłowie zauważyli. I wszystkie te postulaty i nasze odpowiedzi, które postulaty uwzględniliśmy, a których nie i dlaczego, są dostępne w tym dokumencie i można się z nimi zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dodatkowej ochrony, to wydaje się, że przedstawiłem to na samym początku w trakcie prezentowania ustawy.

Rzeczywiście może tego czasu nie było dużo. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dyrektywa, którą implementujemy, została przyjęta w 2014 r. i dostaliśmy mniej więcej 2 lata na implementację tej dyrektywy, tzn. 10 kwietnia 2016 r. ona powinna już być notyfikowana, jak i implementowana. Natomiast kiedy przyszliśmy do resortu, okazało się, że żadne prace nad dyrektywą i jej implementacją nie miały miejsca, dlatego musieliśmy. A przypominam, że przyszliśmy pod koniec 2015 r. Czyli natychmiast jak przyszliśmy, rozpoczęliśmy prace nad tą dyrektywą, bo chcieliśmy zdążyć przed ewentualnymi sankcjami, jakie mogą nas czekać. Jesteśmy na styk, proszę państwa, ponieważ procedura nakładania sankcji się rozpoczęła.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zawarty w druku nr 2232, do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Piotra Walczaka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej przedłożyć projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawowym założeniem rozwiązań zawartych w przedkładanym Wysokiej Izbie projekcie jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Założenie to zostało zrealizowane poprzez szereg działań zawartych w tej ustawie.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w przedkładanym Wysokiej Izbie projekcie należy wskazać zdefiniowanie organów administracji rządowej jako właściwych w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będą nimi jak dotychczas minister finansów oraz generalny inspektor informacji finansowej mający status sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Generalny inspektor otrzymuje dodatkowe uprawnienia w zakresie sporządzania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wydawania decyzji w sprawach wpisu osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, co związane jest z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Wyraźnie wskazano, że jest on także administratorem systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych obejmują nadanie statusu instytucji zobowiązanych nowym kategoriom podmiotów, w tym wspomnianym już podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany walut wirtualnych. Zdefiniowana została na nowo rola komitetu bezpieczeństwa finansowego jako platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym zakresie określono zadania, skład oraz podstawowe zasady funkcjonowania komitetu bezpieczeństwa finansowego. Pozwoli to na zapewnienie rzeczywistego wsparcia generalnego inspektora informacji finansowej w realizowaniu jego zadań. Wprowadzenie obowiązku sporządzania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane oraz określenie mechanizmów sporządzania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na poziomie krajowym, a także działań podejmowanych w celu praktycznego wykorzystania wniosków wynikających z krajowej oceny ryzyka. Proponowane rozwiązania nie stanowią bezpośrednio wdrożenia do projektu ustawy wymogów wynikających z czwartej dyrektywy. Zgodnie z wymogami wynikającymi z czwartej dyrektywy dokonano modyfikacji przepisów dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, w tym wyraźnie zaakcentowano zasady podejścia opartego na ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przy stosowaniu tych środków. Prezentowana ustawa zgodnie z wymogami dyrektywy podstawowy ciężar oceny ryzyka i w związku z tym stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przenosi na instytucję obowiązaną. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ten nowy rodzaj rejestru jest realizacją nałożonego na państwa członkowskie obowiązku ustanowienia go, stanowi narzędzie przeznaczone do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale dodatkowo w związku z objęciem danych gromadzonych w tym rejestrze zasadą jawności służyć powinien także ochronie bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego. Nowelizacja przepisów dotyczy również obszaru pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji przez organy informacji finansowej. Pomimo faktu, że nowe przepisy w tym zakresie nie odbiegają w sposób znaczący od przepisów obecnie obowiązujących, pozwalają na zdecydowanie efektywniejsze wykorzystanie informacji zgromadzonych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez właściwe i uprawnione do tego organy w celu zwalczania innego rodzaju przestępstw. Przygotowano także modyfikację przepisów dotyczących procedury blokady rachunku lub wstrzymania transakcji. Instytucje te stosowane są w związku z podejrzeniami popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ponownie przepisy dotyczące procedury blokady rachunku oraz wstrzymania transakcji w przeważającej mierze powielają rozwiązania funkcjonujące od ponad 15 lat. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wymiany informacji przez organy informacji finansowej z ich zagranicznymi odpowiednikami oraz Europolem. Wprowadzenie tych przepisów stanowi realizację jednego z podstawowych celów, jakiemu służyć miało przyjęcie czwartej dyrektywy. W kontekście międzynarodowego wymiaru, jaki często przybierają schematy przepływu środków związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, umożliwienie pozyskiwania, ale też - co równie istotne - udostępniania informacji partnerom zagranicznym jest zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu. Za istotne należy uznać w prezentowanej ustawie zmodyfikowanie przepisów dotyczące stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom. Dotychczas rozwiązania w tym obszarze związane z funkcjonowaniem komitetu bezpieczeństwa finansowego, jak również legislacyjnym, wydanie rozporządzenia przy współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych pozostawały całkowicie bezskuteczne. Wprowadzono rozwiązania pozwalające na efektywne stosowanie szczególnych środków ograniczających, co pozwoli Polsce jako państwu członkowskiemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych oraz stosowania szczególnych środków, dla których podstawą są rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz decyzje Rady Unii Europejskiej. Dostosowanie przepisów dotyczących kontroli oraz sankcjonowania przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane do wymogów wynikających z czwartej dyrektywy. Proponowane zmiany zakładają depenalizację części zachowań dotyczących przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, objętych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów sankcją karną, a także umożliwiają właściwym organom odstąpienie od nałożenia kary. Prezentowana ustawa zakłada głównie nakładanie kar administracyjnych o charakterze pieniężnym na instytucje obowiązane niewywiązujące się z przestrzegania przepisów niniejszej ustawy. Szanowni Państwo Posłowie! Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Głos ma pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z druku nr 2233.

W toku prac nad tym projektem uwzględniono również zalecenia kierowane przez Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. W art. 1 podano, że ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także inne środki służące ochronie interesu publicznego. W art. 2 wymienione są szczegółowo wszystkie instytucje zobowiązane do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Katalog instytucji obowiązanych wymienionych w tym artykule w znacznym stopniu pokrywa się z katalogiem instytucji obowiązanych określonym w obecnie obowiązujących przepisach. Statusem instytucji obowiązanej objęto, w myśl nowej dyrektywy, przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz spółek i trustów oraz podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi.

Dookreślono zakres definicji podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut. Pozbawiono statusu instytucji obowiązanej przedsiębiorców prowadzących domy aukcyjne, antykwariaty, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi oraz w zakresie sprzedaży komisowej. Z listy instytucji obowiązanych wykreślono również Narodowy Bank Polski, który na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ma specyficzny, dualistyczny status - zarówno instytucji obowiązanej, jak i jednostki współpracującej. Ponadto ograniczono zakres, w jakim adwokaci, radcy prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundamentalne dla projektu ustawy pojęcia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zostały zdefiniowane poprzez odwołanie się do czynów karalnych stypizowanych w Kodeksie karnym. W art. 2 ust. 2 pkt 11 zdefiniowano pojęcie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, wymieniając w lit. b członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów. Intencją projektodawców było objęcie zakresem tej definicji zarówno tzw. kryptowalut, jak i scentralizowanych walut wirtualnych. W rozdziale 2 określono m.in. zadania generalnego inspektora informacji finansowej, zwanego dalej generalnym inspektorem, który podejmuje działania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W rozdziale 3 określono zadania funkcjonowania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. Ustawa, poza przepisami dotyczącymi gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dziękuję bardzo. Głos ma pani poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dostosowanie polskich przepisów do rekomendacji międzynarodowych Financial Action Task Force i do zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Celem zmiany jest także efektywniejsze przeciwdziałanie tym bardzo groźnym zjawiskom w oparciu o dotychczasowe doświadczenia praktyczne w stosowaniu przepisów obecnie obowiązującej ustawy. W związku z dużą ilością zmian, które muszą być wprowadzone do porządku prawnego, rząd zdecydował się na opracowanie projektu nowej ustawy i wydaje się to dobrą decyzją, tym bardziej że pojawia się szereg nowych elementów, nowych rozwiązań, nowych przepisów. Wprowadzane są nowe kategorie instytucji obowiązanych, zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka, wreszcie nowe obowiązki instytucji obowiązanych czy przepisy dotyczące tworzenia, funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Poprawione też zostaną zasady dotyczące generalnego inspektora informacji finansowej i gromadzenia przez niego informacji potrzebnych do wypełnienia nowych ustawowych zadań, a także ochrony zbieranych informacji i procedur, zasad udostępniania tych informacji innym podmiotom. Zmienione też będą przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków. Bardzo ważne jest, żeby te przepisy były precyzyjne, nie budziły obaw uczciwych przedsiębiorców, fundacji czy stowarzyszeń. Wreszcie zmieniane będą też przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na te instytucje. Nowa ustawa ma przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dlatego klub Platformy Obywatelskiej rekomenduje skierowanie projektu do komisji finansów. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Jak tu już wszyscy moi przedmówcy powiedzieli, jest to element realizacji naszych zobowiązań unijnych, wobec tego pewne regulacje musimy wprowadzić do naszego prawa. Musimy.

Cóż, Unia Europejska ma swoją cenę i to jest element tejże ceny.

Tak czy inaczej prace te będą musiały być prowadzone w komisji, dlatego nasz klub będzie rekomendował, aby skierować projekt do komisji i tam podjąć nad nim, nad tym projektem prace. Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Mirosław Suchoń, Nowoczesna. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szanowni Państwo! Ten projekt ustawy ma za zadanie dostosować regulacje prawne do wymogów ujętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jak również do rekomendacji międzynarodowych Financial Action Task Force oraz zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, a także spowodować efektywniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To są absolutnie bardzo, ale to bardzo ważne zadania. Mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo państwa.

Co prawda wiemy, że niewiele państw Unii Europejskiej dostosowało te przepisy, ale to oczywiście nie zwalnia rządu PiS z tego, aby robić to w terminie. Jesteśmy po terminie, panie ministrze.

Państwo mieliście bardzo dużo czasu na to, żeby przygotować te przepisy, a teraz żądacie od parlamentu, żebyśmy tak skomplikowaną materię, która wymaga bardzo dokładnej analizy - zaraz powiem dlaczego - przepracowali w tydzień bądź dwa. To jest niepoważne stawianie sprawy. Tak że apeluję, żeby jednak sprężać się w ministerstwach i przygotowywać przepisy w taki sposób, żeby można je było dobrze rozpoznać w dobrym terminie, tak żeby te przepisy wchodziły z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiście zakres merytoryczny jest bardzo szeroki, więc omówienie tego w takim trybie, jakim jest przedstawienie stanowiska klubu, nie jest możliwe.

Bo wiemy, że w wielu dyrektywach są takie elementy fakultatywne, które można wdrożyć, ale nie trzeba. Kiedy zostaną one wdrożone, powodują dalsze komplikacje. W przypadku wielu wdrażanych do polskiego prawa dyrektyw właśnie takie fakultatywne przepisy zostały wprowadzone. I to jest oczywiście bardzo złe rozwiązanie, tym bardziej że przecież ta ustawa wpływa właśnie na obowiązki, na obciążenia biurokratyczne również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Więc na pewno potrzeba tutaj bardzo szczegółowych wyjaśnień, czy nie ma zbyt daleko idących obostrzeń, właśnie biurokratycznych. Chcę również powiedzieć, że to dobrze, że powstaje nowa ustawa.

Dziękuję bardzo. Głos ma pani poseł Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, druk nr 2233.

Projekt szczegółowo określa instytucje, które są obowiązane do wykonywania obowiązków określonych w ustawie w zakresie wewnętrznego nadzoru. W odniesieniu do administracji rządowej projekt określa instytucjonalnie, kto, w jakim zakresie i w jaki sposób realizuje zadania wynikające z procedowanego projektu ustawy. Organami informacji finansowej w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są minister właściwy do spraw finansów publicznych i generalny inspektor informacji finansowej. Funkcję opiniodawczą i doradczą w tym zakresie sprawować będzie Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, w skład którego wejdą przedstawiciele wielu ministerstw, instytucji i agencji stojących na straży bezpieczeństwa, a także prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. We współpracy z komitetem generalny inspektor dokona krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a następnie opracuje strategię, czyli plan działań mających na celu ograniczenie ryzyka. Wszystkie instytucje obowiązane są zobligowane do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego w bardzo, powiedziałabym, rozległym zakresie dotyczącym m.in. identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości, określenia i monitorowania stosunków gospodarczych, przetwarzania danych o beneficjentach, prowadzenia bieżących analiz przeprowadzanych transakcji, prowadzenia tzw. wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, a także procedury anonimowego zgłaszania naruszeń i informacji przekazywanych generalnemu inspektorowi. Projekt przewiduje również szczegółowe zasady prowadzenia w systemie teleinformatycznym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz zasady przekazywania przez instytucje obowiązane informacji we wszystkich sprawach mogących mieć związek z tym zagadnieniem. Zasadnicza część spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, szczególnie o charakterze decyzyjnym, należy do generalnego inspektora informacji finansowej, którego kompetencje i zakres działań są sprecyzowane w niniejszym projekcie bardzo, bardzo szczegółowo. Projekt ustawy rodzi konsekwencje finansowe, co też jest rzeczą zrozumiałą przy tak obszernym zakresie funkcjonowania ustawy. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w parlamencie, gdzie będziemy mogli, jak sądzę, dokonać analizy, czy nie jest to dokument zbyt biurokratyczny, szczególnie w odniesieniu do instytucji obowiązanych, choć sam cel projektu jest w pełni uzasadniony. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest jednym z istotnych zadań państwa służących ograniczeniu przestępczości i zapewnieniu bezpieczeństwa. Wykrywanie i ściganie przestępczości dotyczącej prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest zadaniem trudnym i wymagającym współdziałania wielu organów i służb państwowych, a także współpracy międzynarodowej. W 2014 r. po przeprowadzeniu przez generalnego inspektora informacji finansowej 2400 postępowań analitycznych do prokuratury skierowano jedynie 170 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. Warto nadmienić, że w okresie objętym kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli, tj. od początku 2013 r. do połowy 2015 r., skuteczność systemu kontroli nad instytucjami, które obowiązane są do rejestrowania transakcji ponadprogowych i podejrzanych, była bardzo niska.

W 2015 r. skala zjawiska prania pieniędzy szacowana była na ponad 17 mld zł, natomiast w postępowaniach karnych zabezpieczono majątek w wysokości 3 mln zł oraz orzeczono przepadek mienia o wartości blisko 100 mln zł, co stanowiło 0,6% wymienionej kwoty. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przy pracach projektowych uwzględniono również zalecenia kierowane pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez komitet ekspertów do spraw oceny środków zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zawarte w raporcie z przeprowadzonej w 2013 r. ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie nowej ustawy. W nowym akcie prawnym znajdą się m.in. przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, przepisy dotyczące wstrzymania transakcji i blokowania rachunków, natomiast zasady współpracy generalnego inspektora informacji finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem są określone bardziej precyzyjnie w porównaniu ze stanem poprzednim. Projekt ustawy nakłada na instytucje obowiązane do realizacji przepisów ustawy obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa, takich jak identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta oraz monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem w przypadku korzystania przez ich klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację.

Przepisy nowej ustawy zakładają, że maksymalna kara pieniężna w przypadku określonych w niej osób prawnych wyniesie równowartość 5 mln euro lub 10% całkowitego rocznego obrotu. Proponowana ustawa przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz do lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań.

Moje pytanie nie wiąże się stricte z przepisami ustawy, ale jest ściśle z nią związane. Chciałabym, żeby pan minister powiedział Wysokiej Izbie, dlaczego od 18 kwietnia 2017 r. przestał być aktywny, dostępny wcześniej na stronie głównego inspektora informacji finansowej, bezpłatny kurs e-learningowy pod takim właśnie tytułem - „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” Stara ustawa, ale także ten nowy projekt, wskazuje, że instytucje obowiązane muszą zapewnić udział pracowników odpowiadających w nich za zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w programach szkoleniowych, tzn., że fundacje, stowarzyszenia, także takie, które opierają się na działalności wolontaryjnej, muszą pracownikom zapewnić takie szkolenie na wolnym rynku, co wiąże się oczywiście z kosztami.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowna Pani Poseł! Oczywiście bardzo słuszne pytanie. Jak najbardziej będziemy chcieli wrócić do tej tradycji, są prowadzone intensywne prace, tylko po prostu tamten kurs niestety się zdezaktualizował. Nam zależy na tym, żeby te materiały, które są zawarte na stronach, jednak były jak najbardziej aktualne, dlatego prowadzimy teraz prace nad aktualizacją i oczywiście ten kurs jak najbardziej wróci.

Dziękuję panu ministrowi. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawarty w druku nr 2233, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 58. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Bardzo proszę, głos ma pan poseł Jarosław Szlachetka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Najtragiczniejszy rozdział wspólnej historii Polaków i Żydów otwiera niewątpliwie II wojna światowa. Sytuacja w moich Myślenicach i powiecie nie odbiegała w żaden sposób od sytuacji w okupowanej reszcie kraju. W 1942 r. Niemcy rozpoczęli realizację planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Masowe egzekucje na wschodzie, które pochłonęły setki tysięcy żydowskich ofiar, trwały już od agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. 6 miesięcy później, na konferencji wysokich funkcjonariuszy nazistowskiego aparatu bezpieczeństwa, administracji i NSDAP w podberlińskim Wannsee zatwierdzono plan wymordowania wszystkich europejskich Żydów. Jedną z części tego planu stanowiła operacja eksterminacji Żydów zamieszkałych w Generalnym Gubernatorstwie oznaczona kryptonimem „Reinhardt” na cześć zabitego przez czeski ruch oporu Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. W Polsce za wszelką pomoc okazaną ukrywającym się Żydom groziła kara śmierci. Był to podstawowy czynnik determinujący zachowania niektórych Polaków w stosunku do żydowskich uciekinierów. Niestety, niejednokrotnie fakt ten stawał się swoistym usprawiedliwieniem, wytłumaczeniem w przypadku np. wydawania ukrywających się Żydów. Oczywiście sprawa ta miała dwa bieguny. Na przeciwległym biegunie stali ci, którzy z narażeniem życia udzielali schronienia żydowskim uciekinierom, niejednokrotnie płacąc za to najwyższą cenę, cenę życia swojego i swojej rodziny.

Są one zbadane i udokumentowane przez lokalnych badaczy, jak np. mgr. Marka Stoszka. W świetle tych faktów szczególnie bolesną sprawą jest przypisywanie przez różne środowiska za granicą, ale niestety również i w Polsce, współodpowiedzialności za holokaust Polsce. W czasie trwania okupacji na terenie naszego kraju nigdy nie doszło do próby stworzenia kolaboracyjnego rządu, co miało miejsce w wielu innych okupowanych państwach. Na terenie Polski działała również wysoko wyspecjalizowana organizacja Rada Pomocy Żydom „Żegota”, angażująca w pomoc obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego wiele środowisk.

Żydom pomagały pojedyncze osoby, całe rodziny i wioski, część ruchu oporu oraz wspomniane już przeze mnie wcześniej specjalnie stworzone do tego celu organizacje, jak Rada Pomocy Żydom „Żegota” czy „Uprawa” - „Tarcza” Apogeum tej kłamliwej i oburzającej kampanii przeciw Polsce jest określenie „polskie obozy śmierci” kolportowane na całym świecie przez różnego rodzaju media i pseudobadaczy. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz odpowiednia edukacja społeczna, prowadzona na każdym szczeblu przez naukowców, nauczycieli i edukatorów w sposób szczególny może przyczynić się do całkowitego wyeliminowania tego kłamliwego i szkalującego naród polski określenia oraz daje jednoznaczny sygnał, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej wobec kłamców i tych, co szkalują dobre imię Polski i Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos ma pani poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Wysoki Sejmie! Akademia im. Jana Długosza to jedna z dwóch głównych uczelni wyższych w Częstochowie. Jej studentami są nie tylko mieszkańcy Częstochowy czy północnego subregionu województwa śląskiego, ale ze względu na wysoki poziom nauczania oraz konkurencyjność kierunków na naszej częstochowskiej uczelni studiują także studenci z całej Polski, a dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dzięki programom międzynarodowym - także studenci z całego świata. O przekształcenie Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet od lat starają się władze uczelni, lokalni samorządowcy, a także parlamentarzyści z różnych opcji politycznych. Rząd Platformy Obywatelskiej i kolejni marszałkowie województwa, zdając sobie sprawę z konieczności ciągłego rozwoju uczelni i wspierając dążenia i aspiracje akademii, nie szczędzili środków na jej rozwój.

Rozumiejąc konieczność spełnienia warunków formalnych otwierających drogę do przekształcenia akademii w uniwersytet, władze uczelni od lat nie tylko rozwijają infrastrukturę i otwierają nowe kierunki, dostosowując je do zmieniającego się przecież rynku pracy, ale także dbają o wysoki poziom kadry naukowej. Dzięki temu uczelnia cieszy się ciągłym powodzeniem wśród kandydatów, a w ogólnopolskich rankingach z roku na rok plasuje się na coraz wyższych pozycjach. Jana Długosza uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.

Jestem przekonana, że minister nauki i szkolnictwa wyższego bez zbędnej zwłoki wyda odpowiednie rozporządzenie. Z pewnością tegoroczni absolwenci byliby szczęśliwi, gdyby mogli otrzymać dyplom ukończenia uniwersytetu. Cieszy mnie, że ten honor spotyka naszą Alma Mater pod rządami pierwszej w historii uczelni kobiety rektora. Cieszy też, że swoje 50-lecie uczelnia będzie obchodziła już jako uniwersytet. Pragnę pogratulować determinacji w dążeniu do celu pani rektor prof. Annie Wypych-Gawrońskiej i jej poprzednikowi prof. Zygmuntowi Bąkowi. Jednocześnie jako częstochowianka i poseł ziemi częstochowskiej dziękuję z całego serca panu premierowi prof. Jerzemu Buzkowi, który od lat wspiera częstochowskie uczelnie, a jak pokazuje przykład Akademii im. Jana Długosza, robi to niezwykle skutecznie. Dziękuję. Głos ma pani poseł Joanna Fabisiak, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czy rzeczywiście leki, których pacjenci nie wykorzystują, muszą być marnowane?

Wiem, że w wielu noclegowniach brakuje leków, ale nie tylko w noclegowniach.

A dlaczego pacjenci leków nie wykorzystują? Bardzo często lekarze wypróbowują, który lek będzie działał najskuteczniej, zatem zmieniają leki.

Nie podaję sposobu rozwiązania tego problemu, bo to nie miejsce i nie czas, natomiast apeluję. Kiedyś z tej samej trybuny, przed wieloma laty, apelowałam o właściwe wykorzystywanie żywności, która jest marnowana.

To bardzo dobrze.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.